Wysoka Izbo! Wnoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o projekty ustaw, które od wielu tygodni leżą w tej Izbie. Po pierwsze, Senat Rzeczypospolitej już dawno zawnioskował o to, by objąć zasiłkami opiekuńczymi również rodziców dzieci do 15. roku życia oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Po drugie, od dawna upominamy się o to, by pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i wsparcie wynosiły 40 tys., a nie tylko 5. Po trzecie, mówimy wyraźnie, że polscy pracownicy powinni być równo traktowani. Nie może być podziału na lepszych i gorszych, nie może być tak, że osoba, która zatrudnia więcej aniżeli 9 osób, po prostu nie otrzymuje tego wsparcia. I wreszcie, panie marszałku, absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której państwo w sposób wybiórczy jedne druki dopuszczacie, a drugie odrzucacie.

Dziękuję bardzo. Panie pośle, senacki wniosek został już rozpatrzony przy okazji tarczy pierwszej. Ale on stał się bezprzedmiotowy w chwili, gdy przyjęliśmy tarczę antykryzysową.

Wysoka Izbo! W tych ciężkich, dramatycznych czasach powinniśmy pamiętać o tych, którzy przysłużyli się Polsce i Polakom. Otrzymaliśmy niestety wczoraj smutną informację, że zmarł radny miejski Jersey City w aglomeracji nowojorskiej, wielki obrońca Pomnika Katyńskiego w tym mieście, wielki przyjaciel Polski i Polaków. Dlatego bardzo proszę, żeby tego człowieka, pochodzącego zresztą ze społeczności koreańskiej, pana Michaela Yuna uczcić chwilą ciszy w Sejmie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Wnoszę o uzupełnienie porządku dziennego o projekt uchwały, który został zgłoszony przez klub Koalicji Obywatelskiej, druk nr 309, w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia. Sejm Rzeczypospolitej wyraża wdzięczność i uznanie dla pracowników ochrony zdrowia za pełną poświęcenia bohaterską służbę w dniach epidemii. W tym czasie lekarki i lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, pracownicy laboratoriów, personel przychodni i szpitali, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, pracownicy socjalni, a także rzesze wolontariuszy ryzykują swoje zdrowie i życie, by nieść pomoc - wierni złożonej przysiędze, a także najlepszym tradycjom polskiej służby zdrowia. Wydaje się, panie marszałku, że nie ma bardziej odpowiedniego dnia, żeby pan uzupełnił porządek dzienny i druk nr 309 dziś został wprowadzony i przegłosowany przez Wysoką Izbę. Szanowni Państwo! To jest wyraz szacunku wszystkich Polaków, panie marszałku, dla pracowników służby zdrowia. Dziękuję bardzo. Mamy następny wniosek formalny. Wysoka Izbo! Zgłaszam się z wnioskiem formalnym o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu wydłużenia czasu na dyskusję nad obydwoma projektami, które mają być przez Wysoką Izbę w tej chwili dyskutowane. Nie kwestionuję uprawnień marszałka i Prezydium Sejmu do połączenia tego, natomiast wyznaczenie limitu 5 minut na dyskusję uważam za dość niecodzienną metodę na kreowanie dyskusji dotyczącej chyba najważniejszego z tematów i problemów, z jakimi nasz kraj się dzisiaj mierzy. Jak mówię, to dobry kierunek, ale 5 minut na dyskusję to zdecydowanie za mało. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie tego wniosku i wydłużenie czasu na debatę do przynajmniej 10 minut. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. No, byłoby bardzo dobrze, gdyby ta dyskusja miała charakter merytoryczny i gdybyśmy rzeczywiście dyskutowali o konkretnych rozwiązaniach. Mamy dwa wnioski formalne o przerwę. Ogłaszam 20 minut przerwy.

Panie pośle, sytuacja jest taka: Prezydium Sejmu czy raczej Konwent Seniorów zwołuje marszałek Sejmu.

Konwentu nie możemy teraz zwołać, natomiast możemy skrócić przerwę.

Bo ja się mogę zgodzić na wydłużenie wystąpień do 7 minut, tak jak wczoraj poszliśmy na kompromis, natomiast przeszlibyśmy do punktów naszego programu i gdyby była potrzeba głosowania, to wtedy będziemy się mobilizować do głosowania.

Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekty to odpowiednio druki nr 330 i 324. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu, oraz w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 7-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Projekt, który Rada Ministrów przedkłada Wysokiej Izbie, jest właśnie takim komplementarnym rozszerzeniem działań przygotowanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mam zaszczyt przed Wysoką Izbą zaprezentować ten projekt i jego najważniejsze założenia. Można powiedzieć, że ten projekt składa się z kilku części. Pierwszą, niewątpliwie dość obszerną, niezwykle ważną, niosącą największe koszty, są kwestie ratowania miejsc pracy, kwestie ratowania polskich firm. W związku z tym zaproponowany zostaje mechanizm wakacji składkowych, czyli zwolnienia z ZUS-u. Dotąd mieliśmy w tarczy antykryzysowej to rozwiązanie przewidziane dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla mikrofirm w odniesieniu do pracowników, a teraz mówimy o pracownikach, którzy są w firmach małych, czyli tych, które zatrudniają od 10 do 49 osób.

Drugą sprawą, niezwykle ważną, jest kwestia umów cywilnoprawnych, umów zlecenia, umów o dzieło.

To jest drugie z rozwiązań.

Dlatego zostały zaproponowane mechanizmy, które mają ułatwić redukcję kosztów, które są możliwe do osiągnięcia już w tym roku budżetowym. Wysoka Izbo!

Chcemy bronić za wszelką cenę miejsc pracy, chcemy ratować polskie firmy i chcemy tak bardzo i tak często proponować zmiany, by można było jak najbardziej elastycznie reagować na potrzeby rynku i na to, co dzieje się dzisiaj w polskiej gospodarce. Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o wsparcie tego projektu, bardzo proszę Wysoką Izbę o pracę nad tym projektem i bardzo proszę Wysoką Izbę, abyśmy mogli pochylić się nad rozwiązaniami, które zostały zaprezentowane. Dziękuję panu ministrowi. Bardzo proszę, pani minister. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

I tak jak wielokrotnie wspominamy i przekazujemy w przestrzeni publicznej, zależy nam na tym, aby te procedury były proste, abyśmy przede wszystkim objęli wsparciem polskiego przedsiębiorcę, każdego pracownika, bo za tymi wnioskami - a chciałabym państwu przytoczyć statystyki, jak one wyglądają na ten moment - stoi konkretna sprawa danej osoby.

Najważniejszy w tym wsparciu jest człowiek, i działania, które rząd podejmuje, są przemyślane, przeanalizowane. Wielokrotnie państwo wspominacie, że ta tarcza nie działa. Nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy sensowne jest ich funkcjonowanie, przede wszystkim powiatowych urzędów pracy, przy malejącym bezrobociu. Dzisiaj statystyki dotyczące bezrobocia za marzec tak naprawdę nie odzwierciedlają sytuacji, jaką za chwilę będziemy mieli w kraju, dlatego nawet tych statystyk nie przybliżam, bo wiemy, że rejestrowanych jest coraz więcej osób bezrobotnych.

Ale my podejmujemy przede wszystkim takie działania, które mają być wyprzedzające, abyśmy zminimalizowali skutki tej tragicznej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Szanowni Państwo! Na ten moment wpłynęło w sumie 340 tys. wniosków.

Mamy złożonych ok. 56 tys. wniosków na postojowe - postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla umów cywilnoprawnych. Na ten moment mamy również złożonych w kraju, i to w każdym powiatowym urzędzie pracy, ok. 31 tys. wniosków na mikropożyczki.

I najważniejsza grupa, którą wspieramy, a więc Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli te środki, które idą na ratowanie konkretnych miejsc pracy, w zależności od tego, czy pracodawca podjął decyzję o postoju ekonomicznym czy też o obniżeniu warunków pracy. Na ten moment mamy złożonych ponad 3,5 tys. wniosków do gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych. Te wnioski są złożone na ratowanie ponad 100 tys. miejsc prac, a przypomnę, że tarcza funkcjonuje zaledwie kilka dni. Jak szacujemy, bo to są szacunki, chociaż pierwsze wypłaty już ruszyły, mamy dzisiaj złożonych wniosków na ponad 700 mln zł, przez te kilka dni.

Monitoruję składanie wniosków, czy w powiatowych urzędach pracy, czy w wojewódzkich urzędach pracy, i każdego dnia spotykam się na wideokonferencji z wojewódzkimi urzędami pracy, a także pani minister Alina Nowak - z powiatowymi urzędami pracy, z ich przedstawicielami. Wnioski są składane on-line. A więc taki instruktaż ekspertów jest na bieżąco przez nas udzielany. Będziemy przede wszystkim dbać o to, aby polski pracodawca, aby każdy pracownik miał ochronę miejsca pracy, abyśmy po tym trudnym czasie, w którym jesteśmy teraz, który zapewne jeszcze będzie trwał, w miarę bezpiecznie i w miarę szybko mogli wrócić do funkcjonowania, które już nie będzie takie, jak przed kryzysem, który jest spowodowany pandemią. Dziękuję, pani minister. Teraz proszę pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy z druku nr 324. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 zaprezentować ustawę o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej. Zanim przejdę do uzasadnienia projektu i jego prezentacji, w Światowy Dzień Zdrowia chcę jeszcze raz, chyba w imieniu nas wszystkich, niezależnie, z której strony politycznej barykady się znajdujemy, podziękować wszystkim pracownikom ochrony zdrowia: pielęgniarkom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, lekarzom, również wszystkim pracownikom administracji szpitali, przychodni, którzy w tych trudnych czasach dbają o nasze bezpieczeństwo. To wy jesteście prawdziwymi bohaterami. To dzięki wam Polska może skutecznie walczyć z koronawirusem. Wy zdajecie egzamin. Niestety nie wszystkie instytucje ten egzamin zdają. Światowy Dzień Zdrowia i nasza prawdziwa tarcza antykryzysowa uzupełniają się w tym zakresie. Zacznę od tej części projektu, która dotyczy wydolności ochrony zdrowia. Żeby poradzić sobie z największym kryzysem, z jakim mamy do czynienia od czasów II wojny światowej, żeby przejść przez kryzys zagrożenia biologicznego, ale również kryzys gospodarczy, musi być kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich sektorów życia społecznego, życia publicznego. Żeby to było możliwe, to najpierw musi być wydolny system ochrony zdrowia. Bez wydolnego systemu ochrony zdrowia nie będzie szansy na uratowanie gospodarki, czyli zaczynamy od rzeczy najważniejszych. System ochrony zdrowia, jak pokazują doświadczenia państw, w których koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie, jeżeli dobrze funkcjonuje, nie tworzy zagrożenia. Jeżeli źle zaczyna funkcjonować, jest przeciążony, niedofinansowany, brak jest odpowiedniej ilości sprzętu zabezpieczającego medyków, przestaje funkcjonować, rozsiewa, staje się źródłem zakażenia, dochodzi do rozsiania się koronawirusa nie tylko na wszystkie inne placówki ochrony zdrowia, ale do jego błyskawicznego rozprzestrzeniania się. Jak usprawnić system ochrony zdrowia i jak zabezpieczyć jego funkcjonowanie? Po pierwsze, 20 mld z funduszy europejskich, również z budżetu państwa, na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu. Czynią to dzisiaj samorządy. Doceniam wszystkie starania, również rządzących, ale 20 mld to jest zastrzyk potrzebny, żeby szpitale mogły funkcjonować, żeby lekarze i pielęgniarki czuli się bezpiecznie, ale też żeby pacjenci, nie tylko zagrożeni zarażeniem koronawirusem, ale też ci, którzy cierpią na inne schorzenia, mieli dostęp do ochrony zdrowia. Ta sytuacja trwa już miesiąc. Pacjenci onkologiczni czekają w coraz dłuższych kolejkach. Wiele oddziałów stoi pustych, więc dzisiaj też trzeba dokonać zmian w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Udało się to osiągnąć, w ostatni weekend to rozporządzenie zostało zmienione. Potrzebne jest monitorowanie oddziałów, które są szczególnie zagrożone, oddziałów interny i geriatrii, gdzie przebywają pacjenci starsi, często 80-, 90-letni. Potrzebne jest monitorowanie domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych i w tych oddziałach dostęp do testów powinien być jak najszybszy. Dodatki dla pracowników ochrony zdrowia, kolejna sprawa, gdyż ich praca jest związana z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, poświęceniem dla całego społeczeństwa, poświęceniem swojego życia rodzinnego. To jest pierwszy dział, który dotyczy utrzymania sprawności systemu opieki zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia. On gwarantuje, że przechodzimy teraz do drugiego. W prawdziwej tarczy antykryzysowej naszego autorstwa jest drugi cały zasób działań związanych z pracownikiem, przedsiębiorcą, pracodawcą, rolnikiem. Wynagrodzenie minimalne powinno być wypłacane we wszystkich firmach, które mają przestój ekonomiczny, poniosły straty. Proponujemy zastosowanie mechanizmu monitorowania tych strat: miesiąc do miesiąca, ale również rok do roku - spadek obrotów o 15% rok do roku lub o 25% miesiąc do miesiąca.

Zasiłek opiekuńczy - była już wielokrotnie mowa o tym na tej sali. Senat nad tym pracował, za co bardzo serdecznie dziękuję, i mogliśmy skorzystać z tego w trakcie prac nad poprawkami, nad ustawą. Zasiłek opiekuńczy do 12. roku życia dla pracowników. Nie może być tak, że różnicuje się dzieci, opiekę nad dzieckiem 8-letnim, a pomija się dziecko 9-, 10-letnie. Powinno być tak naprawdę do 15. roku życia, ale rozumiejąc też głosy strony rządzącej, wprowadzamy rozwiązanie do 12. roku życia. Jeśli chodzi o pracowników odbywających kwarantannę, w tych firmach, w których dochodzi do objęcia kwarantanną pracowników, proponujemy zatrudnienie na zastępstwo i państwo finansuje minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na zastępstwo. To są - część przynajmniej - propozycje dla pracownika. Dla przedsiębiorcy tu jest cała gama rozwiązań. Trzeba pójść bardzo odważnie, trzeba pójść na grubo. Inaczej nie uratujemy polskiej gospodarki, nie uratujemy miejsc pracy. Pani minister mówiła, i słusznie, że wzrasta liczba osób rejestrujących się jako osoby bezrobotne. A więc im więcej zainwestujemy teraz, im więcej włożymy w polską gospodarkę dzisiaj, tym większy będzie zwrot.

A więc to będzie bardzo dobra inwestycja, tylko ona musi być odważna. Fundusz Płynności. Bardzo ważny temat, który dotyczy wszystkich firm. Szczególnie narażone są branże takie jak turystyka, branża transportowa, branża usług. Brakuje pieniędzy na wykonanie podstawowych zadań związanych z prowadzeniem firmy. Jeżeli firma traci płynność, to w szybkim tempie upada. Płynność będzie zachowana tylko i wyłącznie, jeżeli będzie poważna linia kredytowa w Banku Gospodarstwa Krajowego, nieoprocentowana, która da gigantyczne możliwości małej, średniej firmie, mikrofirmie i tej największej firmie, która zatrudnia najwięcej pracowników. Te pieniądze będą przeznaczone na zakup towarów, na zapłatę za usługi, na zapłacenie wynagrodzeń, na wypłatę wynagrodzeń. O tym mówił już wcześniej pan poseł Tyszka, kiedy pracowaliśmy nad pierwszą tarczą antykryzysową. W branży turystycznej od 50% do 70% pracowników już jest zwolnionych, 600 tys. pracowników może być zwolnionych - tylko w tym dziale gospodarki, który odpowiada za 6% polskiego PKB.

Jeżeli oni nie będą mieli Funduszu Płynności, to będą niestety zamykali swoją działalność gospodarczą i nie odrobimy tego szybko. Zwrócili się o pomoc do banków, ale i w tych polskich, w tych, które polonizowaliście, i w tych wielkich zagranicznych zostali potraktowani z buta. Po prostu nie udziela się im kredytów obrotowych, nie udziela się im kredytów pomocowych, tylko są traktowani z buta. Po co są wasi ludzie w tych zarządach, jeżeli nie są w stanie dzisiaj udzielać polskim firmom kredytów? Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Płynności.

Nie ma tych zmian w regulaminie. Wystąpienia - 5 minut.

To jest rozwiązanie, które proponujemy od miesięcy. Teraz trzeba wpisać je na trwałe w polski system, żeby była możliwość dobrowolnego ZUS-u. Odroczenie zaliczek wpłat podatków CIT i PIT dla wszystkich firm. Nie wolno różnicować firm na lepszy i gorszy sort, na te zatrudniające do dziewięciu. Ale tam też tylko połowę bierzecie. Jak firma zatrudniająca 250 pracowników da wszystkim wypowiedzenia, to upada nie tylko ta firma, nie tylko są zwalniani ci pracownicy, ale też upadają mikrofirmy, które z nią kooperują. A więc zwolnienie z ZUS-u, zwolnienie z PIT-u i z CIT-u - to zawiera prawdziwa tarcza antykryzysowa. Rozwiązania dotyczące kredytów i leasingu. Nie tylko wakacje kredytowe, ale wydłużenie raty kapitału oczywiście i raty związanej z odsetkami, ale również wydłużenie okresu spłaty kredytu, żeby nie doszło do kumulacji jesienią, która też, jak wszystkie wskaźniki i wszystkie analizy pokazują, może nie być okresem prosperity. Chorobowe płatne od pierwszego dnia. To jest wielkie obciążenie dla firm, szczególnie w czasie kryzysu, że przez pierwsze 30 dni firma ponosi koszty wypłaty chorobowego dla pracownika. Szybki zwrot podatku VAT. To był jeden z pierwszych wniosków zgłaszanych przez pracodawców, przez przedsiębiorców, że w 3 dni można zwrócić VAT. Będziecie dochodzić i macie już, myślę, ten system weryfikacji bardzo dobrze dopracowany, często się tym chwalicie, więc można dzisiaj zwracać VAT w bardzo szybkim czasie. To są rozwiązania dla przedsiębiorców, pracodawców. Bardzo ważne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Sytuacja jest dramatyczna. Dzisiaj powinny być żniwa dla takich branż jak branża kwiatowa, branża związana ze sprzedażą nowalijek. Oni nie mają gdzie tego sprzedać. Potrzebne jest też wsparcie dla objętych kwarantanną w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Potrzebny jest zasiłek opiekuńczy na podobnych zasadach jak w ZUS-ie wprowadzony w KRUS-ie. Jest zwolnienie z podatku rolnego z rekompensatą dla samorządów. Ale potrzebna jest interwencja na rynku, zakup przez Agencję Rezerw Materiałowych mleka w proszku, masła, ponieważ sytuacja na rynku mleka, na rynku drobiarstwa, na rynku wołowiny robi się dramatyczna. Rynki zagraniczne są zablokowane, nie ma możliwości sprzedaży, nie ma możliwości handlu bezpośredniego. Agroturystyka, zupełnie pominięta w waszych rozwiązaniach, powinna być traktowana jako działalność gospodarcza - choć jest specjalistyczną działalnością rolniczą, ale dotyczy dzisiaj branży turystycznej, która najbardziej ucierpiała. Kolejne rozwiązanie. Prawdziwa tarcza antykryzysowa to zawiera. Nasza propozycja zawiera również rozwiązania ogólne, choćby zablokowanie stosowania dyrektywy, która się nie przyjmie i chyba się nie przyjęła, jest trudna do funkcjonowania w normalnym świecie, a co dopiero w czasie kryzysu. Mówię o dyrektywie dotyczącej RODO. Dzisiaj trzeba ją zablokować, bo ona utrudnia w wielu miejscach wsparcie i pomoc dla pracownika i dla pracodawcy. Szanowni Państwo! Jest szansa na przyjęcie prawdziwej tarczy antykryzysowej. Tylko odwagi. Dzisiaj trzeba być odważnym w działaniu. Sejm ustalił, że w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłucha 7-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dobrze. Przepraszam bardzo. Projekt rządowy przedstawiony przez pana ministra Schreibera, uzupełniony przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej, panią minister Maląg, przedstawia kompleksowe rozwiązanie rozszerzające przepisy związane z tarczą antykryzysową, które weszły w życie zaledwie kilka dni temu.

Tak że z wielkim uznaniem przyjmujemy kolejne rozszerzenie tarczy antykryzysowej przygotowanej przez rząd. Oczywiście oprócz spraw, które są istotne, jeśli chodzi o specyfikę sytuacji, w jakiej w tej chwili żyjemy, czyli takich jak ułatwienia dotyczące choćby zdalnego powadzenia zebrań rad nadzorczych, senatów uczelni itd., co jest dość oczywiste, czyli wzorem Sejmu czy komisji sejmowych - te rzeczy są wprowadzane - to jednak ważne, najważniejsze i najbardziej konkretne wydają się propozycje dotyczące wsparcia przedsiębiorców, wsparcia miejsc pracy. To jest niezwykle istotne, dlatego że za tym stoją bardzo znaczące środki finansowe, takie, które pozwalają na to, żeby te miejsca pracy, może nie wszystkie, ale zdecydowaną większość, uratować.

Niezwykle istotne jest też rozszerzenie kręgu podmiotów, czyli zwiększenie - co już było wspominane - pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających już nie do dziewięciu osób, ale do 49. Jest to niezwykle istotne dla utrzymania miejsc pracy. Bardzo ważnym zadaniem i niezwykle istotnym są pożyczki na utrzymanie miejsc pracy, na podtrzymanie miejsc pracy, pożyczki, które będą podlegały umorzeniu. Oczywiście mowa o pożyczkach, które są obłożone warunkami, czyli zachowania miejsc pracy, ale później z umorzeniem.

Te wszystkie rozwiązania są warte zauważenia i myślę, że w czasie dyskusji będzie można wykorzystać zapisy tego projektu.

Bo chociaż oczywiście cele są szlachetne, to jednak trzeba patrzeć na wszelkie możliwości. Jeszcze ostania rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest opinia Biura Analiz Sejmowych (Dzwonek) do projektu poselskiego, w której zwraca się uwagę, że będzie on wymagał notyfikacji. Oczywiście ten proces notyfikacji prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Teraz w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - pan poseł Dariusz Rosati. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Państwo Ministrowie! Mamy zatem debatować o kolejnym projekcie rządowym dotyczącym walki z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. I to jest już pewna tradycja pracy rządu, ponieważ poprzednie akty prawne były równie obszerne i mieliśmy równie mało czasu. Chciałbym zacząć od prośby pod adresem pana marszałka, aby albo on sam, albo pani marszałek Witek zwrócili uwagę, że w tej sali dochodzi permanentnie do naruszenia elementarnych standardów legislacyjnych. Nie mamy opinii ekspertów, nie mamy opinii Biura Legislacyjnego, nie mamy opinii partnerów społecznych.

Tym razem dostajemy, tak jak powiedziałem, wielki akt prawny, ale w istocie mogę go streścić jednym tylko zdaniem: za mało i za późno. Ponad połowa tego aktu prawnego to są poprawki do poprzedniej ustawy, którą przyjęliśmy tutaj 10 dni temu. W ogóle cały ten projekt aktu prawnego w istocie rzeczy w bardzo niewielkim stopniu przynosi rozwiązania ważne dla przedsiębiorstw i dla pracowników, natomiast w ogromnej części jest poświęcony sprawom proceduralnym, uproszczeniu wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych. Można powiedzieć, że rząd i generalnie administracja państwowa zajmują się w tym projekcie sami sobą. To jest świadectwo braku całościowej koncepcji, to jest też świadectwo swoistej biegunki legislacyjnej, bo to już jest trzecia ustawa, która dotyczy tego samego tematu w ciągu ostatnich 5 tygodni, a bodaj ósma ustawa, która dotyczy walki z kryzysem. Ale co ważniejsze to to, że słyszymy tu, na tej sali, cały czas wezwania do tego, żeby wspólnie pracować nad ustawami, żeby wznieść się ponad podziały partyjne, żeby te ustawy popierać. Chcę powiedzieć, szanowni państwo, że my nie mamy za grosz zaufania do tego, co nam proponuje rząd. 2 tygodnie temu czy 10 dni temu poparliśmy ustawę o tarczy tylko po to, aby zobaczyć, że ostatecznie żadna z naszych poprawek nie została wzięta pod uwagę. Co więcej, pod osłoną nocy rząd wrzucił jeszcze dodatkową poprawkę dotyczącą tematu zupełnie niezwiązanego z walką z epidemią, bo dotyczącą wyborów. Nie mamy do was zaufania. Wielokrotnie nas oszukiwaliście.

Jeszcze raz powtórzę: zwracaliśmy się do Wysokiej Izby i do rządu o poparcie tak oczywistych działań, jak przydzielenie 20 mld zł na wzmocnienie służby zdrowia, jak rozszerzenie zasiłku opiekuńczego na rodziców dzieci do lat 15, potem - lat 12, jak obowiązkowe testy antywirusowe regularnie przeprowadzane w służbie zdrowia w odstępach tygodniowych po to, żeby chronić tych, którzy są na pierwszej linii frontu tej walki. Nie mamy również powodu, żeby wam wierzyć, ponieważ kłamiecie na temat pomocy z Unii Europejskiej. To jest sprawa szczególnie oburzająca, bo nawet Komisja Europejska zwróciła uwagę polskiemu rządowi, żeby po prostu nie przeinaczał faktów, żeby jednak dawał rzetelne relacje co do wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Z tej mównicy padały oburzające słowa o tym, że Unia Europejska nie daje ani 1 eurocenta. Chcę wreszcie powiedzieć, że nie mamy do was zaufania, ponieważ źle ocenialiście sytuację. Mam tu cały szereg cytatów z waszych wypowiedzi, premiera Morawieckiego, ministra Szumowskiego, sprzed miesiąca, sprzed 6 tygodni, kiedy mówiliście, że wszystko jest pod kontrolą, że kraj jest dostatecznie przygotowany, że nic więcej nie da się zrobić. Trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji. Jesteśmy przekonani, że wszystko, co można było podjąć, zostało podjęte - mówił premier Morawiecki 2 marca. 25 lutego szef kancelarii premiera pan Michał Dworczyk mówił: Jesteśmy przygotowani na koronawirusa niezależnie od skali ewentualnych zachorowań. To jest po prostu świadectwo albo tego, że wtedy kłamaliście, albo tego, że nie mieliście zielonego pojęcia, jakie zagrożenia stoją przed Polską.

Dla was wrogiem jest opozycja, dla was podstawowym celem jest utrzymanie władzy i wygranie wyborów. Dlatego nie bierzecie pod uwagę nawet najbardziej oczywistych i zdroworozsądkowych propozycji.

Jest pięć projektów ustaw, które idą w podobnym kierunku jak przedstawiony przed chwilą projekt Koalicji Polskiej, a które są ignorowane przez władze sejmowe i nie są brane pod uwagę przez rząd.

Czy pan poseł złożył wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zresztą dowodów na niedziałanie tarczy antykryzysowej w jej obecnym kształcie dostarczyła obecna tutaj pani minister Maląg. Poinformowała nas ona bowiem, że 340 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski do ZUS-u o różnego rodzaju działania ułatwiające im życie, ułatwiające funkcjonowanie. Czy to jest dużo? To znaczy, że te 340 tys. to jest ledwie co siódme przedsiębiorstwo, co siódma osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą. To jest ledwie 14% wszystkich działających podmiotów gospodarczych. Może już nie działają?

Taka jest prawda, takie są realia, drodzy państwo. Dlatego z nadzieją przypatrywałem się temu, co państwo macie przedsiębiorcom, a zwłaszcza pracownikom do zaproponowania, bo dobry program gospodarczy powinien moim zdaniem mieć następujące cechy. Po pierwsze, powinien być szybki. Po drugie, powinien być prosty. Nasze działania powinny być adekwatne. Po czwarte, ten program gospodarczy nie powinien powodować negatywnych skutków ubocznych. Notabene, panie marszałku, Wysoka Izbo, taki jest właśnie program gospodarczy i propozycje polskiej lewicy, to, co my proponujemy. Proponujemy działania proste, jasne i skuteczne. Proponujemy świadczenia kryzysowe w wysokości płacy minimalnej, czyli 2600 zł brutto, dla wszystkich pracowników, którzy stracili pracę. Proponujemy 50 tys. na pokrycie kosztów stałych na czas kryzysu dla wszystkich przedsiębiorców i dofinansowanie w wysokości, uwaga, 75% pensji pracowników, pod warunkiem że tych pracowników nie zwolnią. Proponujemy wsparcie dla samorządów, bo na nich w tej chwili spoczywa ciężar walki z epidemią koronawirusa. No i oczywiście proponujemy dofinansowanie dla szpitali, w których brakuje sprzętu medycznego i materiałów medycznych. Państwa program, ten pierwszy program, nie spełnia tych kryteriów.

Tak, tu jesteście szybcy. Proponujecie pierwsze - przeforsowaliście, przepchnęliście - drugie, trzecie głosowanie. Gdybyście byli tak szybcy w ratowaniu miejsc pracy, nie byłoby dramatów tysięcy, setek tysięcy pracowników i zamykania tysięcy firm. Wasz pakiet moim zdaniem nie jest także hojny, chyba że za hojność, pani marszałek, panie marszałku, pani minister, uważacie dofinansowanie banków na kwotę 70 mld zł. No to kto leczy z koronawirusa? Banki czy służba zdrowia? Nam się wydaje, że nie banki, ale z podziału środków można odnieść wrażenie, że główny ciężar walki z koronawirusem spoczywa na barkach banków i bankierów. Myślę, drodzy państwo, że nie tędy droga. Zanim ten program tarczy antykryzysowej zaczął działać, już przyniósł skutki uboczne. Są to niestety skutki negatywne.

My jesteśmy gotowi na poważną rozmowę o poważnym programie. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Projekt ustawy przedstawiony przez Koalicję Polską nosi tytuł: o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej. Prawdziwej, bo na tej pierwszej, rządowej, nie można w ogóle polegać.

Dlatego teraz opozycja musi wziąć odpowiedzialność za los Polek i Polaków. I właśnie to czynimy jako Lewica, choć nasz projekt złożony już parę dni temu w Sejmie wciąż nie może doczekać się rozpatrzenia na tej sali. Są w nim dobre rozwiązania, które poseł Robert Kwiatkowski przedstawił w swoim poprzednim wystąpieniu. Projekt Koalicji Polskiej, nad którym w tej chwili debatujemy, zawiera większość tych postulatów. Klub Lewicy poprze skierowanie go do komisji i będzie pracował nad jego rozwinięciem. Na pewno zgłosimy też poprawkę usuwającą dobrowolność składki na ZUS nie tylko podczas epidemii, ale i na zawsze, bo na to Lewica nigdy się nie zgodzi. W czasach pandemii i kryzysu gospodarczego musimy współpracować, zacząć rozmawiać jako politycy z różnych ugrupowań, bo tego oczekują od nas wyborcy. Dlatego też w najbliższych dniach przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski rozpocznie konsultacje ze wszystkimi klubami w sprawie wspólnego projektu uchwały Sejmu o powołaniu komisji nadzwyczajnej do spraw spowolnienia gospodarczego oraz opracowania projektów rozwojowych Polska+. Komisja nadzwyczajna będzie składać się z przedstawicieli wszystkich klubów, ekspertów strony społecznej i rządowej. Dziękuję, pani poseł.

Klub parlamentarny nazywa się Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 i będę bardzo pani marszałek wdzięczny, jeżeli będzie pani podawała prawdziwą nazwę i pouczy pani jeszcze przy okazji pana marszałka Terleckiego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta ustawa mogła być procedowana już wczoraj. Już wczoraj polski Sejm mógł przyjąć rozwiązania tak oczekiwane przez polskich pracowników i polskich przedsiębiorców. Zamiast zająć się jednak prawdziwą tarczą antykryzysową, którą dzisiaj proponuje Koalicja Polska - PSL - Kukiz15, Sejm zajmował się wczoraj przez cały dzień projektem urna+, projektem haniebnym, projektem przeprowadzenia wyborów wbrew woli Polaków, wbrew opiniom lekarzy i wbrew elementarnemu rozsądkowi. Zrobiliście to po to, żeby odwrócić uwagę od problemów polskiej gospodarki. Może podam parę przykładów tego, co wydarzyło się wczoraj.

To, szanowni państwo, jest czubek góry lodowej. To jest początek bardzo poważnej recesji w polskiej gospodarce. Dziś nasza gospodarka krwawi, a wy chcecie nakleić na nią drugi plasterek, proponując pseudotarczę 2.0. Szanowni Państwo! Pracując nad projektem Koalicji Polskiej dotyczącym prawdziwej tarczy antykryzysowej, wsłuchaliśmy się w głos polskich przedsiębiorców i polskich pracowników. Poprawiliśmy waszą dziurawą i tekturową tarczę tak, żeby stała się wreszcie prawdziwą tarczą antykryzysową. Jakie są filary tej naszej prawdziwej tarczy? Pierwsza, najważniejsza, sprawa to zapewnienie firmom płynności. Bez płynności w firmach powstaną zatory płatnicze, a to doprowadzi do fali upadłości i masowych zwolnień. Jedne firmy pociągną za sobą inne. Aby temu zapobiec, proponujemy utworzenie Funduszu Płynności przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Płynności dawałby firmom gotówkę na regulowanie wszystkich zobowiązań o charakterze ciągłym typu najem, leasing, kredyty w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku prosto na konto, w ramach maksymalnie uproszczonej procedury. Szanowni państwo, przedstawiliśmy nasz projekt pani minister Emilewicz już 2 tygodnie temu. Cieszy nas to, że idziecie w tym kierunku, który wskazaliśmy, natomiast już z tych zapowiedzi wynika, że to będzie fundusz biurokratyczny, przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorców. A co z małymi? Drugi fundamentalny punkt naszej prawdziwej tarczy antykryzysowej to dobrowolny ZUS dla wszystkich firm bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów. Zwolnienie z ZUS-u tylko niektórych to jeden z absurdów waszej dziurawej tarczy. To krok w dobrym kierunku, ale nie można różnicować firm ze względu na wielkość, bo czasy są takie, że 95% firm ma problemy.

Trzecia sprawa dotyczy wakacji podatkowych dla przedsiębiorców na kilka najbliższych krytycznych miesięcy. Tego najbardziej brakuje w ramach tarczy 2.0. Firmy stoją teraz przed dramatycznym wyborem, czy zapłacić pracownikom wynagrodzenia, czy czynsz za najem lokali, ratę kredytu, składki na ZUS, czy zaliczki na podatek. Zdejmijmy ten ciężar z firm i zawieśmy pobór wszystkich podatków i opłat na czas epidemii. To powinien być pierwszy krok. W kolejnym kroku, gdy epidemia się już skończy, państwo powinno wprowadzić powszechną abolicję od nieopłaconych podatków i opłat w 30%, 50% lub nawet 100%, w zależności od skali strat firm i sytuacji finansów państwa. Szanowni Państwo! Wasza dziurawa tarcza opiera się na filozofii, jaką w stosunku do przedsiębiorców stosujecie niestety od 5 lat waszych rządów: dołożyć nowy podatek, nasłać kontrolę, stworzyć niejasne przepisy, tak żeby to urzędnik decydował o losie przedsiębiorcy. Do każdego wniosku żądać stosu dokumentów czy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Takie jest wasze myślenie, że skoro w takich warunkach przedsiębiorcy radzili sobie w czasach przed koronawirusem, to poradzą sobie też w czasach koronawirusa. Tylko że ten kryzys jest inny niż wszystkie dotychczasowe i dlatego trzeba zastosować środki nadzwyczajne, proste, automatyczne mechanizmy z biurokracją ograniczoną do minimum. Pomoc powinna być skierowana do wszystkich firm bez kalibracji, bo to nie jest tak, że cierpią jedna czy dwie branże, cierpią mniejsze firmy, a większe jakoś sobie radzą. Cierpią wszyscy, a czas ucieka. Dlatego bardzo proszę Wysoką Izbę o poparcie prawdziwej tarczy antykryzysowej zaproponowanej przez Koalicję Polską - PSL - Kukiz15.

Wysoki Sejmie!

Są takie, które zamrażają w rzeczywistości raty zarówno kapitałowe, jak i odsetkowe, ale są też takie, wśród nich bank, którego prezesem przez lata był premier Morawiecki, które odkładają na później ratę kapitałową, ale żądają dzisiaj spłaty raty odsetkowej. Rata odsetkowa, czasami od kredytu hipotecznego, w połączeniu z koniecznością wypłacania pensji oraz wpłacania przez małe i średnie przedsiębiorstwa również danin (Dzwonek), zwłaszcza do ZUS-u, powoduje, że te przedsiębiorstwa znajdują się na skraju upadku na skutek nie zaniedbań właścicieli czy menedżerów, tylko sytuacji, która została opisana, w wyniku czego ich działalność została ograniczona decyzją ministra zdrowia w rozporządzeniach z 13 i 20 marca tego roku. Dziękuję, panie pośle. Proszę bardzo, pan poseł Jakub Kulesza, Koło Poselskie Konfederacja. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Żeby odegrać z góry ustalone role w tym spektaklu, mylnie nazywanym procesem legislacyjnym? Przed kim i co chcemy dzisiaj udawać? Chcemy udawać, że podejmujemy decyzje? Wczoraj podjęliśmy decyzję o nieuzupełnianiu porządku obrad o nowelizację Kodeksu wyborczego, a za kilka godzin ten kodeks był z powrotem. Udajemy, że tworzymy prawo? Było 39 poprawek zgłoszonych przy pierwszej tarczy przez koło Konfederacja. Wszystkie z automatu zostały odrzucone. Udajemy, że wiemy, nad czym głosujemy? Po wejściu w życie pierwszej tarczy ministerstwa musiały wydać podręcznik liczący 172 strony, który i tak praktycznie niczego nie wyjaśnia. Udajemy, że zapoznaliśmy się z projektem? Na 0,5 godziny przed pierwszym czytaniem wpłynęła treść projektu, tego projektu, który liczy ponad 200 stron, który nowelizuje ponad 60 ustaw. Udajemy, że go przeczytaliśmy, że go przeanalizowaliśmy, że zestawiliśmy z brzmieniem ustaw, że oceniliśmy jego wpływ i teraz bardzo dokładnie zrecenzujemy i zapytamy, czy przypadkiem w nowo dodanym art. 15zzzzzx nie ma błędu w numeracji i czy nie będzie trzeba go poprawiać w tarczy, łacie 3.0? Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Sprawozdawco! Czy państwu nie jest wstyd brać udział w tym przedstawieniu? Czy nie jest głupio tak udawać? Ale przechodząc do rzeczy. prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tak samo porządną gospodarkę i sprawne państwo, i dobre rządy poznaje się w kryzysie. Jaka jest ta Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Premier Mateusz Morawiecki dużo nam obiecywał, jak ta Polska będzie wyglądała. Mieliśmy obietnicę miliona samochodów elektrycznych, dronów, uwaga, mieliśmy mieć przemysł kosmiczny. Zacytuję pana premiera: Będziemy coraz większą pulę środków dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł, w szeroko rozumianym zakresie, i usługi, żeby nasza gospodarka była bardziej nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i praktycznym. No i ta nasza gospodarka, natchniona idealistycznym pierwiastkiem kosmicznym przez pana premiera, na czele ze spółkami Skarbu Państwa, całym tym peletonem, który wiedzie prym w WIG20, z tymi licznymi instytucjami, urzędami, które tak ochoczo państwo powołują z roku na rok, te 7 tłustych lat przejadła, przejadła przez biurokrację, przez klucz partyjny w przyznawaniu stanowisk i przez wyborcze rozdawnictwo. Cała nasza gospodarka przez ten szereg regulacji, wymogów, atestów, cen maksymalnych, które teraz państwo narzucają, nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości tak zaawansowanych kosmicznie technologicznych produktów jak maseczki, jak rękawiczki, nie mówiąc już o bardzo trudnym w produkcji płynie do odkażania. Doszło do tego, że jeden z prezesów spółki Skarbu Państwa został bohaterem narodowym, bo, uwaga, korzystając z przywileju, że urząd właśnie tę firmę zwolnił z konieczności korzystania z atestowanego alkoholu, mógł wyprodukować płyn do odkażania. Oczywiście inne, prywatne firmy nie mogły tego zrobić. Agencja Rezerw Materiałowych nie ma podstawowych wyrobów medycznych, bo, uwaga, musiała kupić węgiel od upadających kopalń ratowanych przez upadające spółki energetyczne. Ale, uwaga, ta sama Agencja Rezerw Materiałowych miała w posiadaniu w połowie lutego, gdy już było wiadomo, jaki nas czeka kryzys w systemie ochrony zdrowia, 63 tys. specjalistycznych, całotwarzowych masek neoprenowych. Miała. Wiedzą państwo, co się stało? 60 tys. maseczek zostało wystawionych na licytacji po 10 zł za sztukę, gdy na rynku chodziły po 130, 140 zł. Oczywiście wszystkie rozeszły się natychmiast, bo ludzie wiedzieli, że jest epidemia, że będą potrzebne, i teraz z kilkudziesięciokrotną przebitką są sprzedawane przez prywatne podmioty. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych też oczywiście nie ma pieniędzy dla zwalnianych pracowników, bo poszły, wbrew założeniu, na świadczenia przedemerytalne. Natomiast wróćmy do tarczy, nazywanej przez was tarczą antykryzysową, a będącej w rzeczywistości betonowym kołem ratunkowym. Jak ta tarcza wygląda? Tak jak mówiłem, nie wiadomo, bo mało kto cokolwiek z niej rozumie. Świadczy o tym ten podręcznik mający 172 strony, który dalej nie wyjaśnia, jak i ustawa, czy zwolnienie z ZUS obejmuje także stronę pracownika, przez co pracodawcy nie wiedzą, jaką wypłacać pensję. Wiadomo za to, że te 5 tys. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających według ustawy mniej niż dziewięciu pracowników, ma nie obejmować tych, którzy nikogo nie zatrudniają. Wiadomo to z informacji, pisma jakiegoś urzędnika, który wbrew ustawie twierdzi, że oczywiście zero jest większe niż dziewięć. Szanowni Państwo! Czego ta ustawa nie zawiera? Przyznam się szczerze, że przez te 0,5 godziny, kiedy miałem tę ustawę w ręku, zdążyłem przekartkować te ponad 200 stron i zauważyć, że ta ustawa nie likwiduje tych 24 nowych procesów biurokratycznych, tych nowych wniosków, nie zwalnia z automatu z narzucanych podatków, opłat, w sytuacji gdy rząd rozporządzeniami wstrzymuje działalność gospodarczą. Czy ta ustawa łata wszystkie dziury pierwszej tarczy? Być może przez te 0,5 godziny, które minie do drugiego czytania, będzie w stanie to ustalić Krzysztof Bosak, który będzie prezentował stanowisko koła w drugim czytaniu. Dziękuję. Zgłosili się posłowie do zadania pytania. Bardzo proszę, 1 minuta, pani poseł. Wysoki Sejmie! Po co komu tarcza nr 2, skoro nie działa tarcza nr 1? Dzisiaj rząd zaprezentował oddziaływanie tej pierwszej tarczy. Otóż za swoje dwa sukcesy uznaliście państwo następujące rzeczy. Sukcesem jest to, że ponad połowa przedsiębiorców planuje skorzystać z tej pomocy. Powiem wam, że ponad połowa tonących chwyta się brzytwy. Niestety oni wszyscy utoną, tak jak przedsiębiorcy, którym proponujecie pomóc w swojej tarczy. Drugim wasz sukces to to, że jesteście w stałym dialogu, a ja powiem wam, że to jest wasza porażka, bo zamiast mówić, trzeba robić. Weźcie pakiet bezpieczeństwa Koalicji Obywatelskiej, który od 2 tygodni leży w Sejmie, i wspólnie uratujmy polską gospodarkę.

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szejna, Lewica. Wysoka Izbo! Wysłuchałem kolejnych propozycji rządu, które są tylko leczeniem za pomocą pudru ciężkiej choroby gospodarczej: pacjent ma wyglądać dobrze, a nie wyzdrowieć. Nie uwzględniliście propozycji Lewicy: 20 mld na dofinansowanie i doposażenie służby zdrowia, dopłaty do kosztów stałych dla przedsiębiorców do wysokości 50 tys. zł miesięcznie, sfinansowania 75% wynagrodzeń pracowników i gwarancji zatrudnienia. Od 1 kwietnia dziesiątki tysięcy przedsiębiorców zawiesiło lub zlikwidowało swoją działalność. Dramatycznie wzrasta bezrobocie. Czy zatem zostaną podwyższone zasiłki dla bezrobotnych? Co zamierzacie zrobić z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który jest pusty? Czy poprzecie sprawiedliwy projekt Lewicy o świadczeniu kryzysowym dla wszystkich dramatycznie dotkniętych kryzysem? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Protasiewicz.

Pani Marszałek! Przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu dostaliśmy 250 stron tekstu, który mieliśmy przeczytać, zanalizować, skonsultować i jeszcze pewnie wyciągnąć wnioski. Przejrzałam oczywiście na szybko ten projekt i stwierdziłam, że jeśli chodzi o oczekiwaną przez przedsiębiorców pomoc, to niestety jej nie ma. Oczekują przede wszystkim natychmiastowej pomocy i wsparcia w utrzymaniu bieżącej płynności finansowej. Że macie państwo zamiar, rząd ma zamiar uruchomić ubieganie się o różne formy wsparcia finansowego. Będą to m.in. pożyczki płynnościowe. Czy na koniec tego ubiegania się niestety nie będzie już firm?

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Mirosława Nykiel, Koalicja Obywatelska. Słyszę, że jeszcze nie ma pani poseł. Ale jest pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Czy rozumiecie, że Austria, Czechy, Dania znoszą te kretyńskie ograniczenia? A wy chcecie je jeszcze pogłębiać. To, co trzeba zrobić, to wrócić do normalności. Nie robimy nic, a wtedy wszystko będzie działało samo. Dziękuję, panie pośle.

Ale dlaczego rząd, pani minister - kieruję teraz te słowa do pani minister pracy, rodziny i polityki społecznej - nie chce pomóc przedsiębiorcom uczciwie, rzetelnie, solidarnie przejść przez ten trudny okres miesiąca, dwóch albo trzech, kiedy ich działalność została niemal wygaszona do zera? Mówię zwłaszcza o tych branżach, których działalność została de facto zakazana rozporządzeniem ministra zdrowia, bez rozróżniania na małe, mikro- i średnie przedsiębiorstwa, bez wyznaczania liczby osób, których ZUS zostaje zawieszony, zamrożony. Dziękuję, panie pośle. Pani Marszałek! Pani Premier Emilewicz! Mniej propagandy, więcej działania dla polskich firm i ratowania polskiej gospodarki. Podam tylko trzy przykłady, jak to wyglądało w marcu na tle trzech innych państw. Kiedy rząd polski proponuje przedsiębiorcom 5 tys. zł pożyczki, i to pod pewnymi warunkami, rząd niemiecki proponuje dotacje do wysokości 15 tys. euro bez zwrotu albo nieoprocentowane pożyczki. Kiedy rząd polski proponuje firmom, które zatrudniają mniej niż dziewięciu pracowników, zwolnienie z ZUS-u, rząd francuski zwalnia firmy z wszystkich danin i pokrywa koszty zatrudnienia.

W dyskusji zgłoszono wnioski: o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk nr 330, oraz o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z druku nr 324. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Wysoka Izbo! Przedstawiciel Platformy czy Koalicji Obywatelskiej powiada rytualne: za mało, za późno, źle itd.

Tak, dokładamy kolejne rozwiązania krok po kroku. Nikt na świecie, i doskonale o tym wiecie, nie był przygotowany na skalę problemu i wyzwania, przed którymi stoimy w związku z pandemią.

W 6 dni, panie pośle. To po pierwsze.

To nieprawda.

Możemy oczywiście rozmawiać w tym momencie o przemyśle kosmicznym, tylko czy naprawdę to jest nasz największy problem? Wysoka Izbo!

Tylko sami sobie państwo odpowiedzcie, czy to jest uczciwe. Oczywiście, nikt nie wpada tu w triumfalizm i nie opowiada, że wszystkie problemy zostają rozwiązane. Jasne, że nie. Jasne, że jest wiele pracy przed nami, ale zestawianie tego poza wszystkim z krajami, które przez 300 lat mogły akumulować swój kapitał, które nie doświadczyły zaborów, które nie doświadczyły komunizmu, to jest naprawdę wyjątkowe. I w tym sensie symptomatyczne jest, że do tej dyskusji z największą troską o przedsiębiorców dwie największe partie wysyłają byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. i to rzeczywiście jest symptomatyczne. Wysoka Izbo! Łączny poziom wsparcia, który został zaprezentowany w tej ustawie, to ponad 11 mld zł. Państwo z Platformy i z Lewicy, którzy zgłaszają wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy po pierwszym czytaniu, mówicie tym wszystkim ludziom, że to są nieważne rozwiązania. Szanuję i rozumiem to, że opozycja przedstawia swoje projekty, ale dlaczego chcecie ten odrzucić, to naprawdę trudno mi zrozumieć. Proszę Wysoką Izbę o odrzucenie tych wniosków. Jeżeli to nie będzie sprostowanie pańskiej źle zrozumianej wypowiedzi, odbiorę panu głos, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek.

Po pierwsze, to wy obiecaliście 212 mld pomocy, a w budżecie zapisaliście 10 mld. To wy odrzuciliście wszystkie merytoryczne poprawki Senatu oprócz tych, które Senat przyjął na wniosek pani minister Emilewicz. My pokazujemy, jak można współpracować. To jest szczyt hipokryzji. Jeżeli pan jeszcze wytacza takie absurdalne argumenty, to tylko udowadnia pan, że to jest pusty dokument, to jest dokument dla urzędników, a nie dla ludzi. Dzisiaj przedsiębiorcy chcą realnej pomocy, chcą tego, co mają w innych krajach Unii Europejskiej, zaś wy proponujecie 10 mld w budżecie, a mówicie o 212 mld. Proszę o zabranie głosu panią Marlenę Maląg, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowni Państwo! Tarcza antykryzysowa, którą przedstawiliśmy tydzień temu, do której wprowadzamy w wyniku przeprowadzonych analiz kolejne zmiany, to jest realnie funkcjonujące wsparcie i funkcjonujące już. Szanowny Panie Pośle!

Przede wszystkim to szerokie wsparcie ma pomóc ochronić miejsca pracy.

Może pozwolę sobie przypomnieć, że jeżeli pracodawca wprowadzi ograniczenie czasu pracy ze względu na to, że jest pracodawcą w kłopotach, do 20%, to również, co w tej ustawie zaznaczamy, może skorzystać z dofinansowania do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

To jest rzeczywista ochrona miejsc pracy, na to pójdą te środki i tych pieniędzy nie zabraknie. Nie zabraknie tych środków również dla pracodawców, którzy podejmą decyzję o przestoju ekonomicznym.

Nie zapomnieliśmy o samozatrudnionych, umowach o dzieło, umowach-zleceniach. To właśnie na tym nam przede wszystkim zależy, aby polska rodzina miała szerokie wsparcie. Dziś wymiar tego programu jest zupełnie inny. W tej trudnej sytuacji, nie sytuacji spowodowanej przez rząd, ale sytuacji, która jest od nas całkowicie niezależna, świadczenie to pozwala dodatkowo wesprzeć polskie rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. Szanowni państwo, bądźmy precyzyjni i posługujmy się danymi. Na dziś bezrobocie nie wzrosło o 500 tys. Dzisiaj nie ma takich danych. My te dane, tak jak państwu powiedziałam, każdego dnia zbieramy, zbieramy je w systemie, nie tworzymy tych danych sami. Jeżeli chodzi o kolejne wsparcie, które na pewno znajdzie się w kolejnej lub jeszcze następnej tarczy, to analizujemy sytuację na rynku. A więc nie zostawimy naszych rodzin bez wsparcia.

Przede wszystkim mają służyć wsparciu pracodawców i pracowników, zachowaniu płynności firm. Te wszystkie mechanizmy są zawarte w tej tarczy, która była przedstawiona tydzień temu. Dlatego też prosimy państwa o wsparcie naszych wspólnych działań, abyśmy przede wszystkim działali w tej trudnej sytuacji - dla każdego z nas, dla każdej rodziny, dla każdego przedsiębiorcy - w zgodzie i porozumieniu i abyśmy podejmowali takie działania, które przede wszystkim będą służyły Polkom i Polakom, i wyszli z tej trudnej sytuacji w jak największym stopniu suchą nogą. Jeszcze raz przypomnę, że w dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk nr 330, oraz o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 324. Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy o godz. 18.45, a teraz zwołuję Prezydium i Konwent Seniorów, Konwent - zdalnie, Prezydium - u mnie w gabinecie. Dziękuję.

Wznawiam obrady. Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów, przedłożyło projekt uchwały w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia, druk nr 331. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego projektu. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia (druk nr 331) Proszę państwa posłów o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i uznanie dla pracowników ochrony zdrowia za pełną poświęcenia bohaterską służbę w dniach epidemii. W tym czasie lekarki i lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, pracownicy laboratoriów, personel przychodni i szpitali, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, pracownicy socjalni, a także rzesze wolontariuszy ryzykują swe zdrowie i życie, by nieść pomoc - wierni złożonej przysiędze, a także najlepszym tradycjom polskiej służby zdrowia. Tak jak wielokrotnie w historii naszego kraju, tak i dzisiaj wobec zagrożenia, przed jakim stanęła nasza wspólnota narodowa, pracownicy medyczni dają najlepszy przykład odwagi oraz heroizmu i stanowią wzór dla społeczeństwa. Jesteśmy wdzięczni wszystkim pracownikom służby zdrowia, przedstawicielom wszystkich zawodów medycznych, a także Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych za pełne zaangażowanie w walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem, za współpracę z instytucjami państwa i samorządu oraz koordynację działań na rzecz społeczeństwa” Proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę przez aklamację.

Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie wyrażenia wdzięczności dla pracowników ochrony zdrowia.

Do głosowania nad tymi wnioskami przystąpimy niezwłocznie. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm podjął decyzję o skierowaniu tego projektu do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy zawartego w druku nr 330, zechce nacisnąć przycisk.

jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Pod głosowanie poddam obecnie wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania poselskiego projektu ustawy. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm podjął decyzję o skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania poselskiego projektu ustawy z druku nr 324, zechce nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?